Wysoka Izbo! Wznawiam posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Bożenę Żelazowską i Daniela Milewskiego, którzy prowadzić będą protokół i listę mówców. Uprzejmie proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów. Panie i Panowie Posłowie!

Odczytam również komunikat o posiedzeniach zespołów.

Dziękuję bardzo. Jesteśmy w bardzo trudnym momencie. Na koszulce mam napis nieprzypadkowy: Achtung Rosja. To bardzo znamienne, choć powinno być: Achtung Putin, ponieważ to on chce skłócić naród rosyjski z demokratycznym światem, którego częścią jest Ukraina. Jestem przekonana, że wyrażam opinię wszystkich tu zgromadzonych, mówiąc stanowcze: nie agresywnym zapędom Putina - Putina mordercy, Putina terrorysty, Putina zbrodniarza. Niech żyje Ukraina! Jesteśmy z tobą, solidaryzujemy się. Ukraina! Precz z Putinem! Ukraina! Precz z Putinem!

Pan poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, Koalicja Polska. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Sytuacja jest dramatyczna, spadają bomby na sąsiednią Ukrainę, są zagrożone życie i zdrowie ludzi, wojna trwa w powietrzu, na morzu i na lądzie.

Białoruś zaatakowała Ukrainę. W obliczu tego oczekujemy w Polsce solidarności i odpowiedzialności sił politycznych i wszystkich obywateli. Zwracam się do wszystkich sił politycznych w Polsce o powściągnięcie emocji, solidarność i odpowiedzialność. Deklaruję gotowość do współpracy i współdziałania. Oczekujemy debaty w parlamencie, oczekujemy zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, oczekujemy wspólnego wystąpienia prezydenta Rzeczypospolitej i wszystkich liderów sił politycznych. Proszę moich rodaków, proszę wszystkich mieszkańców Polski o współdziałanie i solidarność w tym trudnym momencie (Dzwonek), o zaangażowanie wspólnoty samorządowej, o udzielenie pomocy, o współdziałanie z Unią Europejską i NATO, o podejmowanie jak najszybszych decyzji. Nie ma miejsca na błazenadę polityczną, nie ma miejsca na politykierstwo, jest miejsce na solidarność i odpowiedzialność. To jest czas próby obywatelskiej i społecznej. Budowanie - a dzisiaj wręcz odbudowa - wspólnoty narodowej jest podstawową racją stanu Rzeczypospolitej. Tej racji stanu będziemy się domagać, tę rację stanu będziemy prezentować, o tę rację stanu będziemy zabiegać. Polska musi zdać egzamin w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa i pokoju na świecie.

Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, za ten głos. Trzymajmy się czasu, bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dziękuję, pani marszałek, za te słowa, które - jestem głęboko przekonany - płyną z serc nas wszystkich. Dzisiaj pani reprezentowała nas. Rzeczywiście brutalny, bandycki atak Federacji Rosyjskiej i Białorusi na Ukrainę zmienia świat. Nic nie będzie już takie, jakie było. To nie jest wojna interesów. To jest wojna wartości - wartości, na których zbudowane są wszystkie wolne państwa, wszystkie państwa Zachodu.

To jest wreszcie wojna wolności słowa przeciwko państwowemu kłamstwu. Dzisiaj powinniśmy odpowiedzieć bardzo odpowiedzialnie sankcjami, solidarnością i spójnością narodową. To jest wielka odpowiedzialność, która na nas spoczywa w tej Izbie. Dlatego powtórzę apel Szymona Hołowni z przedwczoraj: czas, abyśmy zawarli, wszystkie siły polityczne w tej Izbie, pakt dla bezpieczeństwa. To jest rzecz absolutnie kluczowa. Zastanawiałem się, czy złożyć wniosek formalny z prośbą o poddanie pod głosowanie dodania informacji premiera na temat bezpieczeństwa państwa w tym momencie, ale uważam, że to jest sytuacja tak oczywista, że premier dzisiaj powinien przemówić i że dzisiaj powinniśmy uzupełnić nasze obrady o ten punkt. I jestem przekonany, że pan premier ten wniosek, który płynie z wszystkich ław tej Izby, zrealizuje. Jak pan wie, premier jest cały czas zaangażowany w rozmowy międzynarodowe, we wsparcie dla Ukrainy. Natomiast ważne są w tej chwili rozmowy i w nich uczestniczy premier. Ważniejsze są działania, bo one mogą zatrzymać to, co się dzieje w tej chwili. Bardzo proszę, pan poseł Przemysław Koperski, klub Lewica, wniosek formalny. Dzisiaj czarny dzień w historii, nowożytnej historii Europy. Z taką sytuacją, jaka ma dzisiaj miejsce od rana, nie zetknęliśmy się od kilkudziesięciu lat. Zostały naruszone prawa i integralność naszego wschodniego sąsiada, Ukrainy. Ja z tego miejsca chciałem podziękować bardzo serdecznie wszystkim samorządom w Polsce, które w sposób grupowy, gremialny zadeklarowały wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Chciałem z tego miejsca podziękować bardzo serdecznie wszystkim Polakom, którzy udzielają w tej chwili pomocy naszym przyjaciołom ze Wschodu. Chciałem również powiedzieć, żebyśmy wszyscy dzisiaj byli przyjaciółmi i opiekunami Ukraińców, którzy już są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ale nie zapominajmy również, pani marszałek, o tych Polakach, którzy mieszkają na co dzień na terenie Ukrainy, którzy mieszkają w Donbasie, w Charkowie, którzy mieszkają w Kamieńcu, którzy mieszkają w Kijowie, którzy mieszkają we Lwowie. Zwracam się z prośbą, z wnioskiem formalnym o zwołanie Konwentu Seniorów, żeby przedyskutować kwestię sankcji dla Rosji. Rozmowy się toczą. Pan poseł Cezary Grabarczyk, Koalicja Obywatelska, wniosek formalny. Ja już nie oczekuję, że to będą wnioski formalne, bo sytuację mamy rzeczywiście dramatyczną. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nasz wschodni sąsiad, Ukraina, został zaatakowany przez Rosję. Tam trwa regularna wojna. Od tego momentu świat nie jest już taki sam i Izba powinna też przejść na pracę w trybie nadzwyczajnym. My nie możemy dzisiaj rozpatrywać w tej chwili pytań w sprawach bieżących, tylko powinniśmy zdać egzamin z przywództwa. To miejsce jest najważniejsze w Rzeczypospolitej. Pani marszałek powinna w tej chwili zarządzić przerwę. Powinien się zebrać Konwent Seniorów i powinniśmy ustalić formalny tryb pracy w tych nienormalnych warunkach, ponieważ nie możemy być obojętni (Dzwonek) na to, co dzieje się na wschodzie. Jeżeli padnie niezależna, niepodległa, integralnie bezpieczna Ukraina, zmieni się także bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Proszę nie przejść obojętnie nad tym wnioskiem. Pani marszałek może zarządzić przerwę, skonsultować się z panią marszałek Witek.

Dziękuję bardzo. Dodam, że w tej chwili trwa narada u pana prezydenta w kontekście kolejnych działań. Będziemy państwa informować. Przypominam, że postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 5 minut. Prawo do postawienia pytania dodatkowego przysługuje wyłącznie posłowi zadającemu pytanie. Dodatkowe pytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a uzupełniająca odpowiedź nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu wypowiedzi na pytanie dodatkowe.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Rozwój i upowszechnianie stosowania nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań w ochronie zdrowia to kolejny ważny kierunek strategii Ministerstwa Zdrowia. Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia pozwalają zwiększyć zarówno skuteczność i efektywność leczenia, jak i wykorzystanie zasobów kadrowych czy infrastrukturalnych. Bardzo ważnym kierunkiem w tym obszarze jest rozwój i upowszechnianie rozwiązań łączących elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Należy zauważyć, że także zwiększenie potencjału naukowego sektora ochrony zdrowia jest bardzo istotnym wzmocnieniem i działaniem dla bezpieczeństwa i poprawy jakości leczenia pacjentów. Jakie są możliwości finansowe Ministerstwa Zdrowia do wspierania innowacyjnych rozwiązań w medycynie w celu zarówno skrócenia, jak i polepszenia jakości leczenia pacjenta? Dziękuję. Uprzejmie dziękuję, pani poseł. Na pytania odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan minister Waldemar Kraska. Uprzejmie proszę, panie ministrze. Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Rzeczywiście głos mi się łamie, bo jesteśmy w bardzo wyjątkowej sytuacji, ale musimy dalej pracować.

Pani poseł, jeżeli chodzi o finansowanie i rozwój innowacyjności w medycynie w celu poprawienia jakości leczenia pacjentów, to jest to jedno z priorytetowych działań, jakie jest prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia. Mówimy tu o rozwoju e-zdrowia, ale w tym także telemedycyny. Główne założenia to zapewnienie pacjentowi możliwie najlepszej opieki i dostępu do informacji na temat swojego stanu zdrowia, ale także dostarczenie odpowiedniego wsparcia personelowi medycznemu, poprawienie funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz zwiększenie efektywności, jakości i dostępności udzielanych świadczeń. Ostatni czas, czyli okres pandemii, pokazał, że rozwijanie rozwiązań cyfrowych jest zasadne i pozwala na odciążenie sektora ochrony zdrowia przy zachowaniu odpowiedniej jakości usług. Korzyści, które płyną z rozpowszechnienia innowacyjnych cyfrowych rozwiązań w obszarze zdrowia to m.in. optymalizacja zasobów, korzystny wpływ na zmniejszenie kolejek do świadczeniodawców, lepsza jakość usług poprzez wprowadzenie wysokich standardów oraz zwiększenie dostępu do specjalistów. Przypomnę, że wprowadziliśmy już w roku 2020 e-receptę, tak ważną w okresie pandemii. Receptę, która jest w tej chwili czytelna, nawet jeżeli pacjent ją zgubi, jest do odtworzenia, jest ważna przez cały rok bez konieczności wizyty u lekarza. Zdecydowanie to rozwiązanie sprawdziło się w okresie zagrożenia koronawirusem. To zdecydowanie ułatwiło rejestrację pacjentów w podmiotach leczniczych. Internetowe konto pacjenta. To konto, które służy do bieżącego informowania o zdrowiu pacjenta, o wynikach np. testu na koronawirusa, o przepisanych lekach, o naszych kontaktach ze służbą zdrowia. W tej chwili mamy w Polsce aktywnych ponad 15 mln kont.

Mogli oni być, i byli, monitorowani przez centrum koordynacji, jeżeli ta saturacja była niezadowalająca, był kontakt z opieką medyczną.

Z KPO chcemy wprowadzić trzy centralne usługi cyfrowe: po pierwsze, narzędzia wspomagające analizę stanu zdrowia, po drugie, rozwój algorytmu sztucznej inteligencji, tj. wsparcie dla lekarza, dla podejmowania przez niego decyzji, oraz budowę centralnego repozytorium danych medycznych.

Następnym funduszem, który będzie wykorzystywany, jest Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy.

Dlatego chcemy, aby nasze systemy medyczne były zdecydowanie bardziej zabezpieczone. Pytanie dodatkowe zadaje pani poseł Barbara Dziuk. Uprzejmie proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tu chciałam podkreślić naprawdę istotną rolę, jaką jest element innowacyjności w działaniu w zakresie rozwoju i zastosowania sztucznej inteligencji, zaawansowanych metod analitycznych w obszarze ochrony zdrowia. Bardzo istotnym elementem jest też usługa e-zdrowie - wiemy, że dokumentacja medyczna jeszcze nie funkcjonuje tak jak powinna w systemie cyfrowym. I tu mam pytanie, panie ministrze, jak będzie w najbliższych latach wyglądać podejście do dokumentacji medycznej w tej sferze cyfryzacji, bo to poniekąd usprawni pewnego rodzaju działania zarówno dla pacjenta (Dzwonek), jak i dla wszystkich służb medycznych. Dziękuję bardzo, pani poseł. Uprzejmie proszę, panie ministrze, o udzielenie odpowiedzi. Pani Marszałek! Rzeczywiście do elektronicznej dokumentacji przywiązujemy bardzo dużą wagę, ponieważ zdecydowanie ułatwia ona działanie w systemie, nie tylko jeżeli mówimy o świadczeniodawcy, ale także o rozliczaniu się z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Myślę, że to zdecydowanie usprawni i poprawi jakość zarządzania w ochronie zdrowia. Myślę też, że ten proces przebiega dość płynnie.

Dziękuję bardzo, panie ministrze. Przechodzimy do pytania przygotowanego przez posłów Lewicy w sprawie przygotowania Polski do udzielenia pomocy humanitarnej obywatelom i obywatelkom Ukrainy, utworzenia korytarza humanitarnego, przyjęcia znaczącego napływu uchodźców, jak również przygotowania systemu edukacji na potencjalną konieczność przyjęcia dzieci uchodźców z Ukrainy i włączenia ich w jego funkcjonowanie, zapewnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, opiekuńczego i wychowawczego oraz przygotowania polskich uczniów na współpracę z rówieśnikami z Ukrainy, w szczególności planów Ministerstwa Edukacji i Nauki włączenia w ten proces organizacji pozarządowych specjalizujących się w edukacji antydyskryminacyjnej. Pytanie jest skierowane do prezesa Rady Ministrów. Zmieniła się kolejność.

Wysoka Izbo! Jak konkretnie wyglądają przygotowania rządu do przyjęcia uchodźców z Ukrainy o nieprzewidywanej liczbie, prawdopodobnie miliona lub więcej? Jaki jest konkretny stan przygotowań korytarza humanitarnego przez MSZ i MSWiA? Czy konsulaty polskie w Charkowie, Odessie, Łucku, Winnicy i Lwowie zostaną wzmocnione kadrowo i proceduralnie celem przyspieszenia udzielania wiz humanitarnych? Jak konkretnie poszerzona zostanie kadra Straży Granicznej, która już teraz przy zaledwie 5 tys. uchodźców znad granicy polsko-białoruskiej nie nadąża z procedowaniem wniosków o azyl i ochronę międzynarodową? Jak konkretnie zaplanowana jest logistyka przyjmowania i kwaterowania uchodźców, chwilowego, tymczasowego i docelowego?

Czy Ministerstwo Sprawiedliwości uzgodni z sądami odstąpienie od praktyki automatyzmu stosowania detencji i kierowania uchodźców do ośrodków strzeżonych? Te ośrodki obecnie już pękają w szwach, a warunki w nich są gorsze niż w polskich więzieniach. Brakuje kadry Straży Granicznej, brakuje pomocy psychologicznej, prawnej i medycznej.

Czy przygotowywane jest uelastycznienie procedur w zakresie uzyskiwania pozwoleń na pracę przez uchodźców z Ukrainy? Jaką rząd proponuje politykę integracyjną w tej sytuacji? I jak wyglądają aktualne uzgodnienia z Unią Europejską co do przyjęcia i relokacji uchodźców? Jakie wreszcie są przygotowania Ministerstwa Edukacji i Nauki odnośnie do napływu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do Polski? Jakie uzgodnienia są podejmowane w tym zakresie (Dzwonek) pomiędzy ministerstwem a samorządami, łącznie z niezbędnym w tej sytuacji wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządów? Z upoważnienia prezesa Rady Ministrów na pytanie odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki pan minister Dariusz Piontkowski. Uprzejmie zapraszam, panie ministrze. Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Posłowie! Pytania, które zadawała przed chwilą pani poseł, skierowane są do kilku resortów. Ja jestem w stanie odpowiedzieć na tę część pytań, która dotyczy przede wszystkim edukacji. Natomiast warto podkreślić, że obecnie wszystkie pozostałe ministerstwa przygotowują się na ewentualny rozwój sytuacji na Ukrainie. Dziś ciągle nie wiemy, jakie będą konsekwencje ataku rosyjskiego, także jeśli chodzi o emigrantów czy uchodźców.

Na pewno dojdzie także do wzmocnienia służb, granicy, ale to są kwestie, o których będzie mógł mówić ewentualnie minister spraw wewnętrznych i administracji. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, które ewentualnie mogą pojawić się wraz z uchodźcami z Ukrainy, to polski system prawny przygotowany jest na sytuację zaopiekowania się cudzoziemcami. Już od kilku lat funkcjonują przepisy, które mówią wyraźnie o tym, że cudzoziemcy pojawiający się w Polsce mogą korzystać z tych samych uprawnień co dzieci i młodzież polskie. Są więc zobowiązani do tego, aby wypełniać obowiązek nauki w szkołach obwodowych, rejonowych. W szkołach podstawowych jest obowiązek przyjęcia tych dzieci, w pozostałych szkołach - w zależności od liczby miejsc. Gdyby takich dokumentów nie można było przedstawić, wówczas wystarczy oświadczenie rodziców. Te dokumenty nie muszą być nawet tłumaczone, więc procedura jest bardzo Dyrektor szkoły ma tutaj zasadnicze znaczenie, to on podejmuje decyzję, do której klasy taki uczeń byłby przyjmowany. Będzie to oczywiście zależało od tego, ile lat nauki ma za sobą uczeń, który chce kontynuować naukę w polskich szkołach. Stąd przewidujemy kilka form możliwej pomocy, która może być udzielona na terenie szkoły. Po pierwsze, można przeznaczyć dodatkowe zajęcia z języka polskiego w wymiarze minimum 2 godzin tygodniowo. Podkreślę, minimum 2 godzin, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że zwłaszcza w początkowym okresie warto, aby była to większa liczba godzin.

Mogą się w nim odbywać zajęcia w wymiarze minimum od 20 do 26 godzin, w tym także nauka języka polskiego. Inne przedmioty mogą być również poświęcone przede wszystkim nauce języka polskiego. Utworzenie takiego oddziału przygotowawczego zależy przede wszystkim od decyzji dyrekcji szkoły. My w subwencji oświatowej przeznaczamy dodatkowe pieniądze na wagę, która poświęcona jest tworzeniu takiego oddziału. Dodatkowo można korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia. W tym wypadku, jak rozumiem, chodzi o język ukraiński. Taka osoba byłaby zatrudniona w charakterze pomocy nauczyciela, by ułatwiać kontakt między uczniem czy uczniami ukraińskimi a polskimi nauczycielami. Jeśli chodzi o studentów uczelni wyższych, mamy szeroko zakrojoną autonomię polskich uczelni. Minister edukacji zwrócił się do rektorów uczelni z prośbą, aby korzystali z możliwości, jakie mają już w tej chwili, tak aby móc ewentualnie przyjąć większą grupę studentów, zwolnić ich z opłat. Mamy umowę z Ukrainą o wzajemnym uznawaniu dokumentów, więc nie powinno być jakichś większych problemów, jeśli chodzi o formalne przyjęcie na studia. Zdajemy sobie sprawę, że wśród tych osób mogą być także osoby pochodzenia polskiego. One także mogą korzystać ze szczególnej pomocy, także pomocy materialnej, ze strony poszczególnych uczelni.

Uprzejmie dziękuję, panie ministrze. Pytanie uzupełniające zadaje pan poseł Robert Obaz. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Dość szczegółowo opowiadał pan o możliwościach, jakie dają szkoły, ale dosyć płynnie przeszedł pan, uciekł od tego początkowego pytania, zakładając, że niestety nie wiemy nic, co w tej chwili będzie się działo.

Dziękuję. Bardzo proszę, panie ministrze. Dziś tak naprawdę nikt nie wie, jaka będzie skala tej wojny i jaka ewentualnie będzie liczba uchodźców. Dlatego dziś nikt nie jest w stanie panu konkretnie powiedzieć, czy to będzie 1 tys., 2 tys., 50 tys. czy znacznie większa liczba uchodźców. Ja wiem, że liczby sięgające setek tysięcy czy milionów robią wrażenie, ale my dziś tak naprawdę nie wiemy, jaka będzie skala ewentualnej migracji i uchodźstwa. Rząd przygotowuje się, ma różne plany, stąd te zapytania wojewodów, o których mówiłem na samym początku.

Podobnie będzie także z pomocą udzielaną w celach edukacyjnych, bo przecież ci uczniowie będą trafiali do szkół w tych rejonach, w których będą ośrodki dla uchodźców. Dziś więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć, w których miastach, w których konkretnych gminach czy w których szkołach pojawi się większa liczba uczniów z Ukrainy. Mówiłem także o tym, że ta pomoc finansowa będzie oczywiście zależała od skali. Jeżeli nie będzie to skala zbyt duża, to w ramach tych mechanizmów, które już dziś funkcjonują, w ramach rezerwy subwencji oświatowej będziemy w stanie dodatkowe środki przeznaczyć dla tych samorządów, które będą dodatkowo przyjmowały uczniów pochodzących z Ukrainy. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że dziś już w polskim systemie edukacyjnym uczy się ponad 100 tys. uczniów z Ukrainy - w szkołach podstawowych ok. 30 tys., niespełna 10 tys. w liceach, podobna liczba w technikach, kilkadziesiąt tysięcy w szkołach policealnych i podobnie kilkadziesiąt tysięcy na polskich uczelniach. Mamy więc już za sobą doświadczenia z uczniami cudzoziemskimi pochodzącymi z Ukrainy. Część samorządów ma już duże doświadczenie w szybszej integracji tych uczniów z uczniami polskimi. Oni mają się opiekować każdym uczniem, który trafi do szkoły, w tym także ewentualnie uczniem zagranicznym.

Aby ta pomoc była bardziej efektywna finansowo, w ostatnim roku doprowadziliśmy do wzrostu wagi na utworzenie oddziału przygotowawczego, o którym wspominałem, o 33%. A więc znacznie zwiększyliśmy dofinansowanie tworzenia tego typu oddziałów.

Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie przygotowane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości: Tadeusza Chrzana, Agnieszkę Soin, Filipa Kaczyńskiego i Mariusza Trepkę w sprawie dodatkowego wsparcia na czysty transport miejski z funduszy europejskich. Pytanie jest kierowane do ministra funduszy i polityki regionalnej. Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Tadeusz Chrzan. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Niestety ciągle jeszcze żyjemy w trudnym czasie pandemii, kiedy to różne ograniczenia i obostrzenia dotykają nas wszystkich, dotykają gospodarki, dotykają naszych miast. Chciałem tu zwrócić uwagę, że szczególnie transport miejski bardzo ucierpiał w wyniku pandemii. Wszyscy pamiętamy ograniczenia w wypełnieniu autobusów, wielu pasażerów rezygnowało też z podróży transportem miejskim. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że większość przewoźników, większość spółek utrzymała ofertę przy zmniejszonej liczbie pasażerów. Stąd też pewnie zachodzi taka potrzeba, żeby tę dziedzinę usług, tę dziedzinę gospodarki wesprzeć dodatkowo. Czy w ramach środków unijnych w kończącej się już perspektywie finansowej 2014-2020 - myślę tutaj np. o Programie Operacyjnym ˝Infrastruktura i środowisko˝ - przewiduje pan minister dodatkowe wsparcie na czysty transport miejski? Na pytanie odpowie minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję serdecznie. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani marszałek za słowa wypowiedziane podczas rozpoczynania dzisiejszych obrad. Wiemy doskonale, że w tak trudnym czasie, jakim jest wojna, a szczególnie wojna u naszych najbliższych sąsiadów, kiedy lecą bomby, kiedy to ataki zostały przypuszczone właściwie ze wszystkich możliwych kierunków, bardzo istotne jest wspólne jednoczenie, brak różnic i dążenie do tego, aby taka polityka jedności była bardziej rozpowszechniona. Myślę, że w ramach tych działań również jedność z naszymi sąsiadami z zachodniej strony jest bardzo potrzebna. Polityka spójności jest jednym z tych elementów, które możemy z pewnością wymienić jako obszar tworzenia wspólnoty, dużej wspólnoty europejskiej, która pomaga krajom należącym do Unii Europejskiej przeciwstawiać się różnym przeciwnościom losu. Szczególnie widoczne jest to w tych miastach, jak panowie posłowie, państwo posłowie mówili, w których po COVID-zie również dochodzi do sytuacji, gdy transport jest ograniczony. Wiemy doskonale, jesteśmy tego świadomi, że pandemia spowodowała duże straty w transporcie miejskim. Z naszych informacji wynika, że w początkowym okresie pandemii liczba kursów, liczba pasażerów spadła nawet o 80%. Z tego też względu dokonaliśmy przeglądu szóstej osi priorytetowej Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝, która była dedykowana jako wsparcie dla tego sektora. Nieduża, choć dostępna pula środków pozwoliła nam podjąć decyzję o wsparciu ośrodków wojewódzkich, będących beneficjentami programu operacyjnego, kwotą w wysokości 25 mln zł na każde z miast.

Są to środki, które są kierowane bezpośrednio przez Komisję, a które mają dodatkowo zasilić programy obecnej perspektywy, by wprost służyć wszystkim tym, którzy potrzebują tych środków i tej spójności, o której mówiłem na początku swojej wypowiedzi. Te środki są ukierunkowane przede wszystkim na ekologiczne, cyfrowe inwestycje. Mówimy także o wzmocnieniu sektora transportu miejskiego w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ dodatkową kwotą 70 mln, ale tym razem euro. Przed nami rozmowy z Komisją Europejską na temat szczegółów tego wsparcia. Jeszcze jest jeden szczególnie ważny temat w kontekście odbudowy transportu miejskiego. To też jeden z obszarów, które chcemy wzmacniać.

Są to plany, w których patrzy się na całość mobilności na terenie miasta, a jednocześnie dba się o to wszystko, o jak najwyższą jakość usług, o jak najwyższą jakość życia.

Przeciwdziałanie temu większemu natężeniu ruchu oraz uwzględnienie przepustowości infrastruktury, stawianie na zrównoważony transport czy działania, które mają przede wszystkim pozwolić na jeszcze większe wzmocnienie tej polityki miejskiej, są jednymi z priorytetowych działań w naszym resorcie. Ośrodki wojewódzkie, tak jak mówiłem, które są (Dzwonek) beneficjentami PO IiŚ, już mają możliwość składania wniosków na nowe środki finansowe. Pytanie uzupełniające, dodatkowe zada pan poseł Mariusz Trepka. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dziękuję za tę odpowiedź. Pan podkreślał, że żyjemy w czasie pandemii. Mam taką nadzieję, że ta pandemia w którymś momencie będzie zanikała, a transport będzie zawsze potrzebny mieszkańcom w dużych miastach. Mam dodatkowe pytanie: Czy przewidywane wsparcie z poziomu krajowego dla samorządowych inwestycji właśnie w transport miejski będzie kontynuowane w następnych latach, w perspektywie 2021-2027?

Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam. Wysoka Izbo! Oczywiście w ramach następcy programu ˝Infrastruktura i środowisko˝, czyli programu FEnIKS na lata 2021-2027, zakładamy kontynuację tego programu. Wiadomo, że jest to jeden z kluczowych sektorów z punktu widzenia zrównoważonego transportu.

Z tych środków korzystać będą mogły obszary funkcjonalne miast, czyli przede wszystkim ośrodków wojewódzkich, a także siedem miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych. Dla nas niezmiernie ważne jest to, że wzmocnienie tych funkcjonalnych powiązań będzie kontynuowane, bo w żadnym mieście transport publiczny nie działa w oderwaniu od gmin sąsiednich. Warto też podkreślić, że chcemy, aby te środki finansowe służyły nie tylko aglomeracjom, ale również tym mniejszym miejscowościom, tym wszystkim, którzy mogą skorzystać z tych pieniędzy w ramach nowego programu FEnIKS. To wsparcie będzie również dedykowane interwencji w ramach rozwoju czystego transportu miejskiego, zarówno w tym wymiarze bardziej infrastrukturalnym, jak i w tym wymiarze taborowym, w tym wymiarze cyfryzacyjnym. Mogę również powiedzieć, że chcielibyśmy, aby były z tego finansowane węzły przesiadkowe, np. te najnowsze parkingi typu Park & Ride poza centrami miast, po to aby usprawnić miejskie systemy funkcjonowania naszych sieci transportu, a także miejskie systemy ITS dla uprzywilejowania, usprawnienia usług publicznego transportu miejskiego. Mogę powiedzieć, że w ramach wszystkich działań i realizowanych projektów, które są przedstawione, możliwe będzie też sfinansowanie wydatków związanych z obsługą i integracją usług transportu publicznego, który jest dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników.

Oczywiście niezmiennie możliwe będzie także finansowanie przygotowania planów zrównoważonej mobilności miejskiej przez władze miast i przez podmioty zaangażowane w realizację polityki miejskiej czy metropolitalnej. Chcemy również, aby wybrzmiało dzisiaj - to jest realizowane od pewnego czasu - że dobrze zaplanowana mobilność w mieście będzie z pewnością kluczowym elementem decydującym o wsparciu ze środków unijnych.

Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej przygotowali pytanie w sprawie pokrzywdzonych mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i budynków komunalnych, którzy zostali pominięci w katalogu podmiotów uprawnionych do zmniejszonej taryfy cen za gaz zawartym w ˝ustawie gazowej˝, czyli w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, kierowane do ministra aktywów państwowych. Pytanie zadaje pani poseł Monika Wielichowska. Odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pan minister Karol Rabenda. Jest. Chciałam zapytać, czy rząd ma świadomość, że ustawa gazowa z rekompensatami nie działa, że jest dziurawa, że wdrożył prawo niesprawiedliwe społecznie. Dlaczego rząd nie słucha dramatycznych apeli mieszkańców wielu spółdzielni w Polsce, którzy nie są objęci ochroną, jaką mają zagwarantowaną gospodarstwa domowe w rozumieniu obowiązującej ustawy - Prawo energetyczne? Do dziś nie ma nawet nadanego numeru druku. Na posiedzeniu sejmowej Komisji Aktywów Państwowych nikt nie odpowiedział na nasze pytania, na interpelację poselską też nie odpowiedzieliście. Nie zrobiliście nic, by pomóc wykluczonym z rekompensat ludziom. A każdy dzień, panie ministrze, bez zmiany tej ustawy naraża mieszkańców wielu spółdzielni w Polsce na gigantyczne podwyżki cen ciepła w mieszkaniach. Mam nadzieję, że rząd jest gotowy na pilną nowelizację ustawy gazowej, zanim zaczną się ludzkie dramaty. Odrzuciliście nasze projekty, nie przyjęliście pomocy z Senatu, to przyjmijcie naszą nowelizację. Ona umożliwi pomoc gospodarstwom domowym, ona zrównoważy, wyrówna prawo wszystkich obywateli do ciepłego mieszkania. Żądam od pana podjęcia pracy i naprawienia tego, co zepsuliście. Czeka na to pan Józef, mieszkaniec Nowej Rudy, który ma 92 lata. Rozmawiałam z nim. Pan Józef w lutym płacił 484 zł, a w marcu musi zapłacić 880 zł. Tyle więcej musi zapłacić za ciepło i podgrzanie wody. Z czego ma zrezygnować emerytka pani Halina, też z Nowej Rudy, która za mieszkanie płaciła 630 zł, a teraz musi zapłacić prawie 1 tys. Co pan odpowie paniom Bogumile i Marii i panu Henrykowi? Nie wierzy mi pan? Na pozytywne rozstrzygnięcie czeka też pani Aneta, przedsiębiorczyni, która jest samotnym rodzicem. W panią Anetę najpierw dwukrotnie uderzył tzw. Polski Ład, a teraz jeszcze ponad 50-procentowe podwyżki za ciepło w domu. Mieszkańcy spółdzielni w Nowej Rudzie, Kłodzku, budynków w Polanicy, Ołdrzychowicach, Nowym Tomyślu, Siemiatyczach, Pile, Chełmnie itd. i wielu innych spółdzielni (Dzwonek) też czekają na równe traktowanie, na rekompensaty. Czekają, panie ministrze, na ciepło w mieszkaniach. Przekazuję panu nasz projekt ustawy, który dzisiaj składamy. Dziękuję, pani poseł. Odpowiedzi udziela, jak już wspominałam, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pan minister Karol Rabenda. Zapraszam, panie ministrze. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Przygotowana przez rząd ustawa kompleksowo odpowiada na skutki i ryzyka związane z obecnym kryzysem. Ustawa chroni odbiorców gazu szczególnie narażonych na szok cenowy, a więc gospodarstwa domowe oraz odbiorców wrażliwych. Zgodnie z ustawą ochrona taryfowa objęła w całości dostawy gazu przeznaczone dla celów bytowych. Chodzi m.in. o wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Co ważne, uchwalona ustawa przewiduje dla podmiotów objętych taryfą zamrożenie cen paliw gazowych i gwarantuje stałą cenę gazu na 2022 r. bez względu na wzrost ceny rynkowej w tym czasie. Niestety wprowadzonych ustawą narzędzi wykorzystywanych w przypadku odbiorców indywidualnych oraz grupy tzw. odbiorców wrażliwych nie można zastosować wobec przedsiębiorców, a takimi podmiotami w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców są przedsiębiorstwa energetyczne, ciepłownicze i elektrociepłownie produkujące ciepło systemowe. Z uwagi na przepisy unijne, do których Polska jest zobligowana się stosować, państwo nie może objąć taryfami gazowymi podmiotów prowadzących rynkową działalność gospodarczą, gdyż to działanie byłoby uznane za niedozwoloną pomoc publiczną. Ponadto należy mieć na uwadze to, że ciepłownie i elektrociepłownie w Polsce do produkcji ciepła wykorzystują różne nośniki energii: węgiel, OZE, głównie biomasę, olej i gaz. Udział węgla w 2020 r. wyniósł 68,9%, a gaz stanowił jedynie 10,6% paliw zużytych do produkcji ciepła. Przy tak znaczącym zróżnicowaniu paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła wprowadzenie preferencyjnych warunków cenowych dla paliw gazowych oznaczałoby nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych na rynku. Jedyną odpowiedzią na brak ustawowego zastosowania taryf wobec przedsiębiorców są bezpośrednie działania spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., która wprowadziła obniżki dla odbiorców biznesowych korzystających z cennika: gaz dla biznesu nr 9.

Obniżką są objęci automatycznie wszyscy odbiorcy podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w zmienionym cenniku. Skorzystanie z obniżki nie wymaga od odbiorców podjęcia jakichkolwiek działań, a ceny uwzględniające obniżkę będą automatycznie stosowane przez sprzedawców w rozliczeniach z odbiorcami bez konieczności zmiany umowy.

Należy także zaznaczyć, że istotnym mechanizmem łagodzącym skutki podwyżek cen gazu są również rozwiązania wprowadzone ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Wsparcie przedmiotowym dodatkiem obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Stawki dodatku osłonowego są uzależnione m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym i wynoszą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437 zł rocznie dla największych gospodarstw domowych. To rozwiązanie pozwala skutecznie wesprzeć najbardziej potrzebujące osoby i rodziny, które najmocniej dotknął wzrost cen energii. Będąc świadomym bezprecedensowej sytuacji, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że rząd dokłada i będzie nadal dokładał wszelkich starań (Dzwonek), by ograniczyć negatywne skutki kryzysu energetycznego dla społeczeństwa, a także, na ile jest to możliwe w świetle obowiązujących regulacji Unii Europejskiej, dla podmiotów gospodarczych. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Pan poseł Jakub Rutnicki z pytaniem uzupełniającym. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie ministrze, niech pan spojrzy, to są podpisy, ponad 2 tys. podpisów zdesperowanych mieszkańców pod tym, żebyście zaczęli w końcu działać. Dwukrotnie odrzuciliście naszą nowelizację. Panie ministrze, nie są.

Jeżeli nic nie zrobicie przez najbliższe kilka dni, od marca będzie kolejna podwyżka. Szanowni państwo, Platforma Obywatelska ma gotowe rozwiązanie. Jeżeli nie macie swojego projektu, weźcie nasz. Czas na działanie, szanowni państwo. Pan minister odpowiada na pytanie uzupełniające. Bardzo proszę. Pan minister Karol Rabenda. Panie Pośle! Jeśli chcecie zmiany tego prawa. Jeśli chcecie pomagać ludziom, to przestańcie stosować obstrukcję, zacznijcie pracować w Sejmie. Przestańcie krzyczeć i popierajcie nasze uchwały, które są. Bardzo proszę, pan minister ma głos. Jeśli chcecie pomagać Polakom, mieszkańcom naszego kraju, wspierajcie rząd w ustawach, które zdejmują z nich obciążenia ich rachunków, które nie są spowodowane działaniami rządu, tylko są spowodowane polityką unijną i polityką międzynarodową.

Dziękuję bardzo, panie ministrze. Upominam państwa i proszę o spokój. Przed chwilą, nie wiem, godzinę temu apelowaliście o to, żebyśmy zjednoczyli się w różnych działaniach, więc proszę, trzymajcie się tego, co mówił wasz przedstawiciel. Kolejne pytanie.

Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Od początku roku wielu księgowych oraz doradców podatkowych dwoi się i troi, aby zrozumieć i odpowiednio zinterpretować przepisy największej od lat rewolucji podatkowej, którą obóz rządzący firmuje pod nazwą Polskiego Ładu. Jaki wpływ miała ta zmiana na portfele obywateli, przekonali się już w styczniu nauczyciele, policjanci, strażacy czy emeryci służb mundurowych, których wynagrodzenia czy emerytury niejednokrotnie były niższe o kilkaset złotych. Przekonali się również o tym emerytowani rolnicy pobierający emeryturę z KRUS. Składka na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 9% wysokości świadczenia, w całości została potrącona z kwoty brutto. Co to oznacza dla rolników, którzy otrzymują jedne z najniższych emerytur w kraju? Ich świadczenia zostały obniżone o 100-150 zł. Panie Premierze! Jeśli emerytury rolników wynoszą 1300 zł brutto, to dlaczego my tym emerytom zabieramy blisko 10% świadczenia. Przy tak rosnących cenach żywności, prądu, gazu te 100-150 zł miesięcznie robi kolosalną różnicę. W związku z powyższym proszę pana premiera o odpowiedź na następujące pytania. Dlaczego rząd obciążył emerytowanych rolników dodatkową składką zdrowotną w wysokości 9% świadczenia? Drugie: Czy emerytowani rolnicy, którzy w tym roku otrzymali mniejsze emerytury, mogą liczyć na zwroty podatku, które wyrównają im tegoroczne straty w wypłaconym świadczeniu? I pytanie trzecie: Czy rząd zmieni przepisy w taki sposób, aby osoby samotnie wychowujące dziecko mogły występować o zmniejszenie zaliczki na podatek dochodowy o dodatkową kwotę zmniejszającą podatek w związku z zamiarem wspólnego rozliczenia kwoty dochodów? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Na pytanie odpowie wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Uprzejmie proszę, panie premierze, o udzielenie odpowiedzi. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Myślę, że teza zawarta w pytaniu jest absolutnym kłamstwem. Mówienie o tym, że rząd obciążył dodatkowo emerytury składką zdrowotną 9%, jest absolutną nieprawdą. Jeśli pan nie wie, to może jednak warto porównać rozwiązania dotychczasowe, czyli z roku 2021, i obecne.

Ale - i teraz jest drugi element Polskiego Ładu podatkowego - kwota wolna od podatku do tej pory wynosiła 3888 zł, a teraz wynosi 30 tys. w skali roku. Wobec tego może jednak spróbujmy przeanalizować, jak wyglądało świadczenie emeryta w poprzednim roku, a jak wygląda obecnie. Warto żeby się pan poseł w to wsłuchał. A więc jeśli emeryt miał 1200 zł brutto, tak?

Obecnie w związku z kwotą wolną od podatku 30 tys. zł ta roczna kwota zmniejszenia podatku wynosi 5100 zł. Jeśli przeliczymy to na miesiące, to mamy 425 zł w obecnym roku i 43 zł w roku poprzednim. Oczywiście to nie koniec, bo teraz trzeba porównać składkę zdrowotną.

Łącznie, bo to liczy emeryt, co zostanie w kieszeni, prawda?

Nie otrzymali mniejszych emerytur. chyba że mają dochody z kilku źródeł.

miesięcznie, to właściwie można oświadczenie o niepobieraniu składki złożyć zarówno w jednym organie emerytalnym, jak i w drugim, i w obydwu skorzystać z tej kwoty.

Faktem jest, że to nie jest żadna dodatkowa składka, po pierwsze (Dzwonek), więc teza zawarta w samym pytaniu jest zła, błędna, tylko jest to składka zdrowotna, która rzeczywiście jest nieodliczalna od podatku, ale dzięki kwocie wolnej każdy emeryt zyskuje, w zależności od wielkości, blisko 100 zł czy ok. 100 zł miesięcznie netto, i to mu zostaje. Dziękuję bardzo, panie premierze. Pytanie dodatkowe zada pan poseł Stefan Krajewski.

Mamy do czynienia z wieloma rolnikami, którzy ciężko pracowali i w swoim gospodarstwie, i dodatkowo na etacie.

Pani poseł, proszę nie przeszkadzać. Ja pani poseł nie będę przeszkadzał, jak pani będzie pytać. Jak pomóc tym rolnikom?

Jeśli jest tak dobrze, to dlaczego ubóstwo na wsi ciągle rośnie?

Zapraszam, panie premierze, do udzielenia odpowiedzi. Panie Pośle! Ta wypowiedź to już naprawdę. Odsyłam pana na zebranie, spotkanie z rolnikami, z emerytami na wsi. Niech pan posłucha, co oni naprawdę myślą o waszych czasach, kiedy to podnieśliście wiek emerytalny do 67 lat i kobietom, i mężczyznom, o tym, jakie były minimalne emerytury, choćby rolnicze, za waszych czasów.

Naprawdę, panie pośle, radzę, żeby jednak dokładnie przyjrzał się pan wyliczeniom.

My mówimy, że emeryci dostają więcej netto, a pan mówi, że mniej. To proszę jechać w takim razie do jakiegokolwiek emeryta rolniczego i zobaczyć jego pasek, jego wypłatę i się przekonać. Nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć, naprawdę. Bo to są kłamstwa. Mówię to jasno i wyraźnie: to, co pan mówi, to są kłamstwa.

Dziękuję bardzo, panie premierze. Przechodzimy do kolejnego pytania.

Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady pomimo bardzo optymistycznego tytułu dotyczącego przeciwdziałania wylesianiu i degradacji lasów jest w rzeczywistości przeniesieniem całości kompetencji w zakresie gospodarki leśnej do Komisji Europejskiej. W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie ma postanowień o wspólnej polityce leśnej Unii Europejskiej, a więc polityka leśna i jej kontrola należą do kompetencji państw członkowskich. W roku 2021 Unia Europejska opracowała nową strategię leśną UE 2030, która zawiera wiele kontrowersyjnych założeń, przeciwko którym protestują środowiska naukowców, praktyków, leśników w całej Europie, przedstawionych m.in. na konferencji w Warszawie w dniu 8 października 2021 r. Tekst projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wskazuje na realne zagrożenie dla polskiego modelu gospodarki leśnej. Projekt rozporządzenia stanie się realnym narzędziem do zawłaszczenia przez prawo Unii Europejskiej prawa do determinowania gospodarki leśnej przez demokratycznie wybranych przedstawicieli kraju członkowskiego. W ten sposób można spowodować blokadę gospodarczą prawidłowo działających podmiotów poprzez żądanie wykonania bezprawnych i niemerytorycznych działań oraz spełnienia nacechowanych ideologicznie oczekiwań wąskich grup społecznych. Mając powyższe na uwadze, zwracam się z pytaniem: Jak Ministerstwo Klimatu i Środowiska ocenia opisany. projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz czy ministerstwo opracowało już stanowisko lub pracuje nad przygotowaniem stanowiska w sprawie tego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, tak aby wypracowane rozwiązania ogólnounijne wspólnych problemów. Na pytanie odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pan minister Edward Siarka. Uprzejmie proszę, panie ministrze. Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo Posłowie! Wysoka Izbo! Rzeczywiście dokument, o który państwo dzisiaj pytacie, jest bardzo ważnym dokumentem, który jest kolejnym przykładem rozwiązań bardzo mocno ingerujących w kompetencje państw narodowych. Dlatego też projekt stanowiska rządu w sprawie przedmiotowego projektu rozporządzenia został już opracowany w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w ścisłym kontakcie i w ścisłych konsultacjach z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, ministrem rozwoju i technologii oraz ministrem finansów, a więc z resortami, które są właściwe dla problematyki, którą porusza to rozporządzenie. Muszę powiedzieć, że Polska bierze bardzo aktywny udział w pracach nad tekstem rozporządzenia, tekstem, który rodzi przecież bardzo dużo pytań.

Przede wszystkim nie zgadzamy się, aby projektowane rozporządzenie ingerowało w zrównoważoną gospodarkę leśną. To nie pierwszy raz, kiedy Komisja Europejska bardzo mocno ingeruje w zrównoważoną gospodarkę leśną, próbuje odebrać kompetencje państwom narodowym w zakresie leśnictwa. Uprzejmie dziękuję, panie ministrze. Proszę o trzymanie się czasu, będę wyłączać mikrofon, bo chciałabym jeszcze punkt przerobić. Jedno pytanie. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź panu ministrowi, ale chciałabym doprecyzować jeszcze to pytanie.

Ponieważ rozporządzenie zakłada kategoryzację krajów na trzy grupy, chodzi o art. 27 w powiązaniu z art. 10, uprawnienia do klasyfikacji krajów będzie miała Komisja Europejska.

Jakie zabezpieczenia przed dowolnością kategoryzacji, dla przykładu - skargi NGO, proponuje wprowadzić ministerstwo? Panie ministrze, proszę o udzielenie odpowiedzi. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Tak jak powiedziałem, to rozporządzenie, gdyby w tej wersji zostało przyjęte, wywoływałby bardzo daleko idące skutki gospodarcze dla takich państw jak Polska. Bo przypomnę, że jeśli idzie de facto o produkty drzewne, a zwłaszcza o przemysł meblarski, to Polska jest na pierwszym miejscu pod względem produkcji mebli, a jeśli idzie o produkt krajowy brutto, to stanowi on prawie 2,5% naszego produktu krajowego brutto. Wszystko to, co jest związane z gospodarką leśną, i - co ważne - 9% całości naszego eksportu to są produkty drzewne. To jest wielka branża, która zatrudnia pół miliona ludzi.

Gdyby Unia Europejska wprowadziła taką listę - bo Komisja Europejska w świetle tego rozporządzenia taką listę chce wprowadzić i ona ma decydować, które państwo na tej liście się znajduje, a które nie - to, proszę zwrócić uwagę, nawet w odniesieniu do tego, co obecnie dzieje się chociażby w Europie, można by bardzo skutecznie wyeliminować Polskę z tego rynku, na którym dzisiaj skutecznie konkurujemy.

I to dotyczy nie tylko produktów drzewnych, lecz także produktów cukierniczych, czekoladowych, piekarniczych czy mleczarskich, ponieważ wszystkim tym produktom można zarzucić w pewnym momencie - czy znajdzie się jakaś grupa ekologiczna czy NGO, która to stwierdzi - że są one produkowane w sposób sprzeczny z zapisami tego rozporządzenia. Bardzo mocno się temu sprzeciwiamy.

Kto o tym będzie decydował? Według jakich procedur?

Pytanie przygotowane przez posłów Koalicji Obywatelskiej w sprawie kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej podejmowanych przez Radę Ministrów na arenie międzynarodowej, w tym szczególnie na forum Unii Europejskiej, NATO, OBWE, oraz krajowych w związku z agresją Federacji Rosyjskiej przeciw Ukrainie, kierowane do wiceprezesa Rady Ministrów. Proszę o trzymanie się czasu, bo za chwilę mam Prezydium i muszę ogłosić przerwę. Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Panie i Panowie Posłowie! Historia tak sprawiła, że to dzisiejsze pytanie jest pewnie najważniejszym pytaniem, przed jakim staje Wysoka Izba. Jest to pytanie o bezpieczeństwo naszych sąsiadów, ale w istocie jest to szukanie odpowiedzi na to, jak zapobiec wojnie. To nie jest ich wojna. To nie jest wojna gdzieś daleko. To jest także nasza wojna. Został podpalony dom naszego sąsiada. Dlatego pierwsza sprawa to powiedzieć dzisiaj Ukraińcom, a być może jutro Gruzinom i innym naszym siostrom i braciom na Wschodzie, że drzwi do Unii Europejskiej i NATO są dla nich otwarte. Oczekujemy tego od polskiego rządu i oferujemy wsparcie w tej sprawie. Oni walczą za nas, oni dzisiaj potrzebują usłyszeć, że ich miejsce jest z nami. I sprawa kluczowa dla każdego polskiego obywatela: dzisiaj ludzie pytają o swoje bezpieczeństwo. Musimy się zjednoczyć, żeby zapewnić bezpieczeństwo każdej polskiej rodzinie. To znaczy, że pytania brzmią: Jak rząd jest przygotowany do obrony przed dywersją? Jak zostało przygotowane wojsko? Ile zostało przeprowadzonych narad? Jakie szczegółowe działania podejmowała Rada Bezpieczeństwa Narodowego, komitet, który odpowiada za bezpieczeństwo? To są pytania, przed którymi stoi dzisiaj każda polska rodzina. A więc będziemy mówić bez wytchnienia. Polacy potrzebują dzisiaj więcej bezpieczeństwa. To wymaga wielkiej mobilizacji na arenie międzynarodowej i na arenie krajowej. I będziemy mówić bez wytchnienia: spokój, ale sankcje i solidarność (Dzwonek), aktywny rząd i wielka synergia wszystkich Polaków, którzy dzisiaj mają na sercu dobro naszej ojczyzny. Odpowiedzi na pytanie udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pan minister Paweł Jabłoński. Bardzo proszę, panie ministrze, i dziękuję, że jest pan z nami mimo tej trudnej sytuacji.

Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Jak państwo doskonale wiecie, śledzicie państwo wydarzenia międzynarodowe, doskonale zdajecie państwo sobie sprawę z tego, że Rosja dziś nad ranem, po raz ostatni, miejmy nadzieję, przekroczyła granice, o których przekraczaniu my mówiliśmy już od wielu, wielu miesięcy. Można było usłyszeć wiele głosów, że te działania zbrojne są tylko straszakiem, są tylko groźbą, że Rosja się nigdy do tego nie posunie. W rzeczywistości niestety stało się tak, jak polski rząd i rządy innych krajów Europy Środkowej, które doskonale to zagrożenie rozumieją, ostrzegały, tak jak my ostrzegaliśmy. Niestety dochodzi do scenariusza najczarniejszego, ale myślę, że za życia nikogo w tej sali nie było jeszcze tak poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa. Polski rząd w tej sprawie podejmował działania od wielu miesięcy. Już w ubiegłym roku, kiedy jeszcze wszyscy skupieni byli na sytuacji bezpieczeństwa dotyczącej naszej wschodniej granicy z Białorusią, my zaczęliśmy dostrzegać, że podejmowane są także pewne działania ze strony Rosji, ze strony Federacji Rosyjskiej: gromadzenie wojsk i na terytorium przy granicy rosyjsko-ukraińskiej, i na terytorium Białorusi. Już wtedy premier Morawiecki spotykał się bardzo intensywnie z przywódcami wszystkich państw Unii Europejskiej, informował o tym, że takie zagrożenie narasta, że trzeba podjąć zdecydowane działania. Dziś jesteśmy w sytuacji, w której część tych działań została już wdrożona, inna część została zapowiedziana. Dziś wieczorem w Brukseli odbędzie się zwołany na wniosek premiera Morawieckiego szczyt Rady Europejskiej, nadzwyczajny szczyt poświęcony właśnie tej sytuacji. Już przez ostatnie godziny trwają bardzo intensywne rozmowy w sprawie tego, jakie sankcje powinny zostać wprowadzone, część z nich została ogłoszona dziś rano przez przewodniczącą Komisji Europejskiej. To jeszcze oczywiście wymaga zatwierdzenia na szczeblu Rady Europejskiej, to jeszcze wymaga jednomyślności wszystkich państw członkowskich.

Takie głosy słyszeliśmy jeszcze w ubiegłym tygodniu z największych państw Unii Europejskiej. Na szczęście dzisiaj, po wczorajszej zapowiedzi kanclerza Niemiec, w końcu zaczyna się to zmieniać. Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest koniec, że nadal różnego rodzaju stronnicy Putina będą podejmowali tego rodzaju kroki, że będą starali się doprowadzić do tego, aby te decyzje za jakiś czas odwrócić. Dlatego tak ważna jest konsekwencja, dlatego tak ważna jest jedność. Bardzo dziękuję za ten głos, za deklarację, że opozycja w tej sprawie będzie wspierać rząd, bo w tej sprawie rzeczywiście wszystkie siły polityczne powinny mówić jednym głosem. To jest interes Polski, to jest interes Europy Środkowej, to jest interes całej Europy, całego naszego kontynentu. Rzeczywiście konieczne jest wsparcie dla naszych sąsiadów, dla naszych partnerów, dla naszych braci na Ukrainie. To wsparcie jest przygotowane. Nasze służby dyplomatyczne, nasze służby konsularne pozostają na miejscu. My oczywiście jesteśmy gotowi do tego, żeby w razie potrzeby podjąć działania ewakuacyjne, ale przede wszystkim chcemy być na miejscu, żeby służyć naszym obywatelom, którzy są na Ukrainie, którzy tam też potrzebują pomocy. Dziś rano zostały zaktualizowane po raz kolejny komunikaty. Zachęcamy każdego, kto tylko może, żeby jak najszybciej rozpoczął działania w celu opuszczenia terytorium Ukrainy. Nasze służby konsularne będą w tym pomagały. Działania, które my podejmujemy, mają tak naprawdę na celu przede wszystkim doprowadzenie do tego, żeby była jedność sojusznicza.

Natomiast jeżeli będziemy jednością jako Zachód, jeżeli będziemy jednością i będziemy zdecydowani, to naprawdę jesteśmy silniejsi, naprawdę mamy instrumenty, których możemy użyć. Dziś wieczorem premier będzie zachęcał wszystkich pozostałych przywódców Unii Europejskiej do tego, żeby na użycie tych instrumentów była gotowość. Bo nie ma się co oszukiwać: cały czas różnego rodzaju stronnicy Putina będą starali się tę jedność rozbijać, opowiadać, że sankcje nie są skuteczne, że sankcje są bardziej bolesne dla Europy niż dla Rosji. To jest nieprawda. To jest nieprawda, trzeba o tym pamiętać. Trzeba te działania kontynuować i polski rząd będzie to robił. Pytanie uzupełniające, pan poseł Sławomir Nitras. Musimy rzeczywiście wszyscy sobie z tego zdawać sprawę. Panie ministrze, dziękując panu za obecność, chciałbym z tego miejsca zaapelować do premiera, do rządzących Polską: To jest moment, w którym musicie dać Polakom poczucie bezpieczeństwa. Bo jak słusznie powiedział pan poseł Kowal: to nie jest ich wojna. Dzisiaj wszystkie polskie rodziny, matki, dzieci wstały rano i zadały sobie pytanie, co mamy robić, jak się w tej sytuacji zachowywać.

Dziękuję bardzo. Pan minister Paweł Jabłoński. Za chwilę ogłosimy przerwę. Pani Marszałek! Państwo Posłowie! Oczywiście taka gotowość jest potrzebna i musimy dziś Polakom dać nie tyle poczucie bezpieczeństwa, co bezpieczeństwo. Dlatego ja również zwracam się z apelem do wszystkich sił politycznych, do wszystkich partii, które mają wpływ także na swoich koalicjantów w innych partiach europejskich, żeby rozmawiać, żeby oddziaływać, żeby pokazywać, że współpraca gospodarcza, energetyczna z Putinem, to, do czego doprowadziliśmy jako Europa - nie chcę tu wskazywać palcem na konkretne państwa, ale wszyscy doskonale wiemy, o kim rozmawiamy. Budowa kolejnych gazociągów doprowadziła do sytuacji, która pozwoliła Putinowi finansować działania zbrojne, których dziś jesteśmy świadkami. To był potężny błąd. Przyznają: byliśmy zbyt łatwowierni. My w Polsce nie byliśmy łatwowierni, my w Polsce mówiliśmy bardzo jasno: to jest błąd, to jest niebezpieczne. Sami kręcimy sobie jako Europa sznur na szyję. Potrzebna jest dzisiaj konsekwencja w rozmowie z tymi politykami, którzy mają realny wpływ na to, jak funkcjonuje Unia Europejska, na to, jak funkcjonuje Europa, jak funkcjonują największe państwa, bo to w tych państwach jest klucz do rozwiązania tego kryzysu. Jeżeli będziemy zjednoczeni, jeżeli będziemy w stanie wprowadzić sankcje, i to takie, które rzeczywiście będą dla Rosji odczuwalne - a możliwości są, natomiast brakuje czasami woli politycznej - jeżeli wola polityczna się pojawi. To jest kolektywne, zbiorowe zadanie nas wszystkich, żeby naszych partnerów w Europie do tego przekonywać. Jesteśmy w stanie to zrobić. Apeluję o to, żebyśmy w najbliższych dniach skupili się przede wszystkim na tym. Spory wewnętrzne, które są między naszymi obozami politycznymi, są czymś oczywistym w kraju. Na zewnątrz tych sporów być nie powinno, bo po prostu tego wymaga nasze bezpieczeństwo. I mam nadzieję, że takich zbędnych, szkodliwych sporów będziemy unikali, a razem będziemy pracować dla bezpieczeństwa Polski, Europy i dla bezpieczeństwa naszych braci Ukraińców.